Dzień dobry państwu. Wznawiam posiedzenie. Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję posłów Filipa Kaczyńskiego oraz Konrada Frysztaka, którzy prowadzić będą protokół i listę mówców. W pierwszej części obrad sekretarzem będzie pan poseł Konrad Frysztak. Bardzo proszę posła sekretarza o odczytanie komunikatów. Dzień dobry. Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji: - Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach - o godz. 9, - do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych - o godz. 9.30, - do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych - o godz. 10, - Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - o godz. 10, - Kultury i Środków Przekazu - o godz. 10, - Sprawiedliwości i Praw Człowieka - o godz. 10, - do Spraw Unii Europejskiej - o godz. 11.30, - do Spraw Kontroli Państwowej - o godz. 12, Infrastruktury wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - o godz. 12.30, - do Spraw Kontroli Państwowej - o godz. 13.30. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panu posłowi. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 11. porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Przypominam, że postawienie pytania nie może trwać dłużej niż 2 minuty, zaś udzielenie odpowiedzi nie może trwać dłużej niż 5 minut. Prawo do postawienia pytania dodatkowego przysługuje wyłącznie posłowi zadającemu pytanie. Dodatkowe pytanie nie może trwać dłużej niż 1 minutę, a uzupełniająca odpowiedź nie może trwać dłużej niż 3 minuty. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu odpowiedzi na pytanie dodatkowe. Przechodzimy do pytań. Zaczynamy od pytania pana posła Waldemara Andzela w sprawie przyjęcia programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027. To pytanie jest skierowane do ministra funduszy i polityki regionalnej. Odpowie na nie sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej pan minister Waldemar Buda. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko to następca dwóch edycji wcześniejszego programu ˝Infrastruktura i środowisko˝ 2007-2014 oraz 2014-2020.

Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Panie ministrze, zapraszam uprzejmie. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Pani Minister! Szanowni Państwo! Program FEnIKS - rzeczywiście to jest jego nowa nazwa, w skrócie, chodzi właśnie o Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

Jest to program, z którego będą mogły korzystać instytucje, podmioty, które będą do niego aplikowały. To są środki, szanowni państwo, które odpowiadają na trzy cele polityki, ale, mówiąc prostszym językiem, odpowiadają na zapotrzebowanie kilku sektorów. Przede wszystkim jest to sektor energii, sektor środowiska, sektor transportu, sektor kultury i zdrowia. Z tych środków buduje się drogi, z tych środków buduje się kolej, z tych środków realizuje się program ˝Czyste powietrze˝, z tych środków realizuje się program ˝Mój prąd˝ - oczywiście między innymi.

W poprzedniej perspektywie - to też warto podkreślić - na ten cel było przeznaczonych 460 mln euro, w tej perspektywie zaproponowaliśmy 700 mln.

Na transport, drogi - 4,5 mld, kolej - 5,5 mld, transport intermodalny - 230 mln, oczywiście euro, transport morski - 760 mln euro, śródlądowy - 220, lotniczy - 50, nawet lekko jest to zwiększone ostatnią decyzją w tej sprawie w ramach konsultacji, które prowadziliśmy jako ministerstwo funduszy. Jest to bardzo ambitny plan, trzeba jasno powiedzieć, że on realizuje bardzo ambitne cele. Możemy się z nimi zgadzać, możemy nie, ale to są bardzo ambitne cele klimatyczne Unii Europejskiej.

Część będzie fazowanych, część etapowanych, ale one będą realizowane w obecnej perspektywie. Program - jak wszystkie inne, krajowych mamy kilka - jest przygotowywany teraz na etapie po złożeniu go oficjalnie 5 stycznia do Komisji Europejskiej. Komisja ma 3 miesiące na ocenę tych programów.

Jesteśmy po konsultacjach międzyresortowych, po konsultacjach społecznych. Oczywiście jeśli chodzi o pieniądze, przesuwaliśmy między poszczególnymi kategoriami, chociaż tutaj trzeba powiedzieć, że pewnej swobody, całkowitej dowolności nie ma, bo marker cyfrowy, marker klimatyczny to było dla nas zobowiązanie wynikające z rozporządzeń.

Myślę, że w I połowie tego roku on będzie już zatwierdzony przez Komisję i będziemy przygotowywać konkretne inwestycje pod ten program. Dziękuję serdecznie. Proszę o pytanie dodatkowe, panie pośle. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo!

Zresztą infrastruktura i kolejowa, i drogowa, i lotnicza to wielkie wyzwanie i na pewno tutaj to dopingujemy. Proszę, panie ministrze. Szanowni Państwo! Program CPK to rzeczywiście jest nowe zadanie, które pojawia się w tej edycji programu, i ono będzie bardzo intensywnie wspierane.

Ale bardzo mocno chcemy je finansować, oczywiście z tego programu.

Co to oznacza?

My mamy tylko pewne ograniczenia czasowe. Co do zagłębia, województwa śląskiego, to oczywiście jest tak, że możemy spojrzeć na statystyki i być spokojni. To znaczy udział województwa śląskiego w korzystaniu ze środków krajowych poprzednika, jakim był program POIiŚ, jest ponadproporcjonalny w stosunku do całego kraju, jeżeli chodzi o liczbę ludności. W związku z tym spokojnie można się spodziewać, że ilość inwestycji, jaka będzie kierowana z tego programu na rzecz województwa śląskiego, będzie adekwatna, będzie proporcjonalna.

Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do następnego pytania. Posłowie Piotr Adamowicz oraz Arkadiusz Myrcha zadadzą pytanie w sprawie wywłaszczenia cennego manuskryptu znajdującego się w posiadaniu Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu i nieodpłatnego przekazania rządowi Węgier. W tej sprawie będzie odpowiadała podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pani minister Izabela Antos. Bardzo proszę pana posła Piotra Adamowicza o zadanie pierwszego pytania. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Od niemal 500 lat dziedzictwo kulturowe Torunia współtworzy niezwykle cenny średniowieczny manuskrypt, który od 1923 r. należy do Książnicy Kopernikańskiej. Dzieło to nie jest łupem wojennym, jak to często bywa. Zostało kupione przed wiekami przez toruńską radę miejską. Otóż niespodziewanie obóz PiS wpadł na pomysł wywłaszczenia tego dzieła, zabrania z Torunia i nieodpłatnego przekazania rządowi Węgier, premierowi Orbánowi. Jak podkreślają naukowcy, z perspektywy światowej rękopis ten jest najcenniejszym kodeksem w kolekcji Książnicy, a jednocześnie jednym z najcenniejszych zachodnioeuropejskich rękopisów iluminowanych z XV w., jakie mimo wielkich, katastrofalnych zniszczeń zachowały się w zbiorach polskich. Projekt przekazania tego zabytku orbánowskim Węgrom wzbudził zrozumiałe protesty nie tylko w środowisku toruńskim. Zgadzam się ze stwierdzeniem, że jest to próba zagarnięcia bezcennego dziedzictwa kulturowego Rzeczpospolitej. W pełni też zgadzam się ze zdaniem toruńskich radnych, że ten skandaliczny projekt może nie tylko próbować pozbawić Toruń części historii, ale także stanowić niebezpieczny precedens odbierania samorządom ich własności. W związku z tym uprzejmie proszę o odpowiedzi na następujące pytania. Kto i kiedy, z jakiego upoważnienia rozpoczął rozmowy z Węgrami w sprawie zabrania z Torunia i przekazania Węgrom tego bezcennego zabytku? Dlaczego wybrano drogę wywłaszczenia przez państwo obiektu znajdującego się w posiadaniu instytucji samorządowej? 25 mln rekompensaty, odszkodowania, które ma rząd zamiar przeznaczyć, to ponad 6 mln dolarów (Dzwonek) Za 6 mln dolarów na rynku antykwarycznym można nabyć bardzo ciekawe rzeczy, nie trzeba ich zabierać polskim samorządom, a w szczególności miastu Toruń. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, pani minister. Zapraszam na mównicę. Dzień dobry. Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie Posłanki i Panowie Posłowie! Szanowni Państwo!

Jest to jedna z dwóch najlepiej rozpoznawalnych zbroi dziecięcych na świecie, jak również jedyna pełna zbroja króla polskiego w obecnych zbiorach Rzeczpospolitej. W wyniku zawirowań historycznych znalazła się ona w Budapeszcie, jednak dzięki osobistym staraniom premiera Mateusza Morawieckiego, który zwrócił się do premiera Węgier Viktora Orbána z oficjalną prośbą o przekazanie renesansowej zbroi, powróciła ona na Zamek Królewski na Wawelu. Nie byli zobligowani do zmiany przepisów zakazujących wywożenia dóbr kultury poza granice kraju. Nie byli również zobligowani do uszczuplenia swoich zbiorów. Byli za to silnie przekonani, że miejsce tego cennego zabytku, a warto tutaj wspomnieć, że jego wartość rynkowa szacowana jest na ok. 12 mln zł, jest w Polsce, dlatego przekazali go Polsce w formie darowizny, bezkosztowo. Gest premiera Orbána był widocznym znakiem przyjaźni łączącej oba narody, a także wyrazem szacunku dla naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego. Węgrom będzie wyrazem wdzięczności za to, że zdecydowali się zwrócić nam unikatowy zabytek bez względu na koszty i wysiłek, do jakich byli zobligowani. Manuskrypt w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu to renesansowy poemat o bibliotece króla węgierskiego Macieja Korwina żyjącego w II połowie XV w. Była to jedna z pierwszych humanistycznych bibliotek królewskich w Europie. Jej ogromne zbiory zostały prawie doszczętnie zniszczone podczas najazdów wojsk tureckich na Węgry w 1526 r., a jej fragment trafił do Polski. Manuskrypt zapisany na 62 kartach jest ważnym źródłem do badania historii biblioteki Korwina. Dzięki niemu można odtworzyć zawartość kolekcji utraconej przez Węgrów. Wartość historyczna i symboliczna, jaką kodeks przedstawia dla narodu węgierskiego, odzwierciedla wartość, jaką ma dla nas zbroja Zygmunta Augusta. Towarzyszy nam przekonanie podobne do tego, jakie mieli Węgrzy, oddając nam zbroję, że ten zabytek związany jest z tożsamością narodową Węgrów i powinien wrócić do ich ojczyzny. Muzeum Narodowe w Budapeszcie nie otrzymało rekompensaty finansowej za zbroję, którą otrzymała Polska. Jesteśmy jednak świadomi, że przekazanie Węgrom ˝Kodeksu Macieja Korwina˝ uszczupli zasoby Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, dlatego podmiot będący właścicielem manuskryptu otrzyma z części budżetu państwa, której dysponentem jest szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, środki finansowe, rekompensatę w wysokości 25 mln zł. Kwota ta odzwierciedla nie tylko cenę rynkową kodeksu, ale także jego wartość historyczną i symboliczną. Kwota rekompensuje także uszczerbek, jaki spowoduje utrata własności kodeksu i wyodrębnienie go z kolekcji bogato iluminowanych rękopisów Książnicy Kopernikańskiej. Przez kraje Europy Środkowowschodniej przez stulecia przetaczały się wojny, przez które utraciliśmy wiele dóbr kultury. Polska, Węgry i inne państwa regionu utraciły sporą część swojego dziedzictwa, bez którego nie jest możliwe budowanie tożsamości narodowej. Staramy się także wspierać w tym dziele inne narody. Nasz gest wobec Węgier jest tego najlepszym wyrazem. Bardzo proszę o pytanie dodatkowe pana posła Arkadiusza Myrchę. Proszę bardzo.

Nie ma problemu. Proszę bardzo. Marnie słychać. A może by pan podszedł, panie pośle, do mównicy?

Pani Minister!

Ze smutkiem to przyznaję, bo jednak dzisiaj debata toczy się nie dla naszej trójki, nie dla parlamentarzystów, tylko przede wszystkim dla obywateli, dla mieszkańców Torunia. Mieszkańcy Torunia, którzy są dzisiaj naprawdę, proszę wierzyć, oburzeni propozycją przedstawioną przez parlamentarzystów PiS-u, nie usłyszeli żadnego uzasadnienia, dlaczego mają zapłacić tak ogromną cenę i czy tylko dlatego, żeby pan premier Orbán miał dowód wdzięczności pana premiera Morawieckiego. Ponad 500 lat ten wyjątkowy zabytek był własnością naszego samorządu, był własnością Gimnazjum Akademickiego, któremu rada miasta prawie 500 lat temu przekazała ten zabytek. Przetrwał on wiele zakrętów naszej historii: przetrwał wojnę, przetrwał komunę, przetrwał zabory, ale okazuje się, że po prostu może nie przetrwać rządów PiS-u.

O tym też dzisiaj nie usłyszeliśmy, dlaczego jest taka wartość, kto ją wycenił. Jaka jest wartość zabytku, który jest od kilkuset lat związany z historią nie tylko Torunia, ale naszego państwa? Dziwi nas to, że polski rząd, który mieni się rządem patriotycznym, chce w sposób dobrowolny pozbawić Polskę, pozbawić polskich mieszkańców, pozbawić mieszkańców Torunia czegoś wyjątkowego, czegoś, co jest integralną częścią naszej narodowej historii tak naprawdę w imię tego, żeby premier Morawiecki poczuł się dobrze i mógł poklepać po ramieniu pana premiera Morawieckiego. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, pani minister.

Przedstawione przeze mnie informacje są informacjami, które posiada Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w zakresie procedowania nad poselskim projektem ustawy, o którym jest dzisiaj mowa. Natomiast odniosę się jeszcze do kwestii wyceny. Skąd kwota 25 mln? Taka kwota została przedstawiona nam, jako dysponentowi części budżetu, szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i zabezpieczona w środkach.

W grudniu 2012 r. sprzedano go za 6,2 mln dolarów.

Przechodzimy do następnego pytania. Posłanki Wanda Nowicka oraz Magdalena Biejat zadadzą pytanie w sprawie wsparcia rodzin będących w trudnej sytuacji ekonomiczno-społecznej w opiece nad noworodkiem, w tym kwestii odbierania dzieci rodzinom, które są w stanie sprawować opiekę nad swoim dzieckiem. To pytanie jest zadane prezesowi Rady Ministrów. Odpowie, z upoważnienia prezesa Rady Ministrów, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej pan minister Stanisław Szwed. Bardzo proszę panią posłankę Wandę Nowicką o zadanie pytania. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Zwracam się z pytaniami dotyczącymi sytuacji rodzin będących w trudnej sytuacji ekonomiczno-społecznej, a które mimo to chcą i są w stanie zajmować się swoimi dziećmi, jeżeli otrzymają niezbędną pomoc ze strony państwa. Pytanie wywołała nagłośniona ostatnio przez media sprawa pani Patrycji, matki karmiącej piersią, której wyrokiem sądu odebrano córeczkę Julię w 3 dni od jej narodzin bezpośrednio ze szpitala św. Zofii w Warszawie wyłącznie na podstawie jednego faksu. Choć sytuacja ekonomiczna rodziny jest niewątpliwie trudna, a rodzice mają orzeczenie o lekkiej niepełnosprawności, to w ocenie osób znających tę rodzinę, gdyby ci rodzice otrzymali niezbędną pomoc, byliby w stanie opiekować się własnym dzieckiem.

Co więcej, bardzo niepokoi sposób, w jaki kobieta została potraktowana przez instytucje, które przejęły opiekę nad dzieckiem. Proszę o odpowiedź na następujące pytania: W jaki sposób służby, których zadaniem jest wspieranie rodzin wymagających pomocy, wspomagają rodziny znajdujące się w trudniejszej sytuacji ekonomiczno-społecznej, aby mogły one sprawować opiekę bez szkody dla dziecka, jeśli oczywiście chcą i są w stanie tę opiekę sprawować? Czy ta pomoc, którą państwo zapewnia, jest wystarczająca? Czy sposób, w jaki została potraktowana pani Patrycja, jest standardem postępowania w podobnych sytuacjach, czy wypadkiem przy pracy? Przypominam, że po pierwsze, odebrano jej dziecko, nie informując o decyzji sądu, po drugie, ograniczono jej dostęp do noworodka, i po trzecie (Dzwonek), uniemożliwiono jej karmienie piersią. Ile jest w Polsce przypadków odbierania dzieci rodzinom w trudniejszej sytuacji, które jednak mają szansę na sprawowanie opieki nad swoimi dziećmi po otrzymaniu niezbędnej pomocy? Podkreślam, że nie chodzi o rodziny, w których występują ewidentne patologie, czyli przemoc, narkotyki, alkohol. Czy w sprawie pani Patrycji rząd podjął działania interwencyjne, kontrolne czy naprawcze w celu sprawdzenia, czy wszystko odbyło się w zgodzie ze standardami? Czy nie jest potrzebna interwencja w tej sprawie? Jeśli takie działania zostały podjęte, to czy są już jakieś ustalenia w tej sprawie? Czy rodzina pani Patrycji otrzymała pomoc ze strony odpowiednich służb? Dziękuję, pani posłanko. Bardzo proszę, panie ministrze. Pan minister Stanisław Szwed, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Witamy pana ministra miło. Panie Marszałku! Pani Poseł!

Jak pani poseł słusznie zauważyła, decyzję podejmował niezależny sąd. Pytanie było tak sformułowane, że zostało skierowane do naszego ministerstwa i stąd moja obecność tutaj.

Ponad 6 mln prawie 600 tys. dzieci w tym programie uczestniczy.

Najświeższe rozwiązanie to rodzinny kapitał opiekuńczy.

Tu akurat już jest kryterium dochodowe - 1922 zł.

Jeśli chodzi o część pytania dotyczącą odbierania dzieci, które przeżywają trudności, to przypomnę, że wprowadziliśmy bardzo zasadnicze zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Bardzo proszę panią posłankę Magdalenę Biejat o zadanie.

Wydaje mi się, że będziesz musiała podejść do mównicy i skorzystać z rady naszej ulubionej pani posłanki z Platformy Obywatelskiej. Panie Ministrze! Oczywiście popieramy te wszystkie programy dofinansowujące rodziny w różnym stopniu, ale nie o to było pytanie.

Już kończę, panie marszałku. Mamy problem dotyczący wsparcia nastoletnich matek, zwłaszcza w przypadku tych, które są w placówkach opiekuńczych i ośrodkach resocjalizacyjnych. W tej sprawie wielokrotnie interweniowali kolejni rzecznicy praw obywatelskich i nic się nie dzieje. Podobno pojawił się projekt, co prawda znowu w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale liczę, że ministerstwo rodziny również się interesuje tym tematem i wie, co się z nim dzieje, który miał tę sprawę rozwiązać, ale utknął w konsultacjach. Czy ministerstwo rodziny interesuje się nastoletnimi matkami, czy trzymacie się zasady, że każecie nam rodzić, a potem radźmy sobie same. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, bardzo proszę. Panie Marszałku! Oczywiście te wszystkie dane, które państwu przedstawiłem, są w bardzo ograniczonej formie, bo też czas na odpowiedź mam bardzo krótki.

Jeśli chodzi o kwestie związane z asystencją, to w 2020 r. zatrudnionych było ponad 3824 asystentów rodziny.

Docelowo chcemy, aby w każdym powiecie był taki asystent rodziny.

Jeżeli mówimy o samorządzie, to bardzo ważna jest rola zarówno samorządu powiatowego, jak i gminnego, żeby w tym zakresie też udzielać wsparcia.

Bo to też jest bardzo ważne w takich trudnych sytuacjach i to w ramach programu ˝Za życiem˝ jest.

Dziękuję serdecznie.

Tak? Dziękuję serdecznie. Panowie posłowie Andrzej Grzyb i Marek Sawicki zadadzą pytanie dotyczące kosztów zawarcia umowy dotyczącej funkcjonowania Kopalni Węgla Brunatnego Turów. To pytanie zostanie zadane prezesowi Rady Ministrów, w imieniu którego odpowie, z jego upoważnienia, minister klimatu i środowiska pani minister Anna Moskwa. Bardzo proszę, panie pośle. Pani Minister! Zostało zawarte porozumienie pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Czeskiej o współpracy w zakresie odnoszenia się do skutków na terytorium Republiki Czeskiej wynikających z eksploatacji Kopalni Odkrywkowej Węgla Brunatnego Turów. Umowa ta zakłada, że Polska ma zapłacić 35 mln euro rekompensaty, natomiast fundacja Polskiej Grupy Energetycznej ma przekazać 10 mln euro krajowi libereckiemu.

Warto zaznaczyć, że 12 lutego 2021 r. ówczesny minister spraw zagranicznych Czech Tomasz Petrziczek przed złożeniem skargi do TSUE zaproponował polubowne załatwienie problemu na przylegającym do kopalni obszarze po stronie czeskiej.

Ważny punkt porozumienia dotyczy również czasu obowiązywania tej umowy, który wynosi 5 lat. Nie można zapomnieć też, że na Polskę została nałożona kara 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego - ja tutaj się nie odnoszę co do zasadności nałożenia tego środka tymczasowego, jak również konsekwencji dla polskiego systemu energetycznego - i polski rząd deklaruje, że nie zamierza płacić tej kary, której wysokość wynosi w chwili obecnej (Dzwonek) 68 mln euro. Chciałbym zadać pytania. Po pierwsze: Do jakich inwestycji zobowiązała się Polska w umowie zawartej z Republiką Czeską?

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani minister. Zapraszam uprzejmie, witając w Sejmie. Panowie Posłowie zadający pytanie! Zanim opowiem o tych inwestycjach, kilka zdań odniesienia się do wstępu w wystąpieniu pana posła. Rzeczywiście ze strony czeskiej padały w toku rozmów bardzo różne propozycje, w tym bardzo różne propozycje finansowe, z tym że trzeba pamiętać, że ta pierwsza propozycja, która się pojawiła w lutym poprzedniego roku, to była propozycja pod tytułem: płacicie środki i na chwilę obecną temat jest zamknięty. To nie była kompleksowa umowa, taka, jaka jest zawarta na dzień dzisiejszy, czyli w żaden sposób nie zabezpieczała nas przed takimi sytuacjami, że w przyszłości Czesi znowu będą mieli kolejne roszczenia, kolejne żądania. W żaden sposób nie określała ona sposobów rozstrzygania sporów potencjalnych, czyli, w domyśle, sytuacja analogiczna albo potencjalny spór przed TSUE mogłyby się pojawić. To była krótka bardzo propozycja na zasadzie: kwota i zakończenie tematu na chwilę obecną. Dodatkowo ta umowa nie była w żaden sposób sparametryzowana ani doprecyzowana - właściwie to nie była umowa, to była propozycja - w zakresie monitorowania. Czyli nadal Czesi, potencjalnie, mogliby mieć roszczenia w związku ze złą interpretacją czy z brakiem danych dotyczących jakości wody, powietrza czy hałasu. To, na czym nam zależało - żeby umowa, którą podpisaliśmy, była umową docelowo, kompleksowo, jednoznacznie rozwiązującą ten spór.

Czyli tak naprawdę będziemy realizować wszystkie inwestycje już określone w decyzji środowiskowej, bo duża część tych parametrów monitoringowych i inwestycji monitoringowych już została określona w decyzji środowiskowej, a to, co jest nowe, to uczestnictwo strony czeskiej. A więc będzie ekspert w momencie, kiedy będziemy wybierać otwór, np. otwór do monitorowania wody - cztery takie otwory są zaplanowane.

Co jest jeszcze istotne, ta umowa jest dwustronna. Na dzień dzisiejszy my też nie mieliśmy od strony czeskiej precyzyjnych informacji co do ich sposobu monitorowania, co do parametrów tego monitorowania. Ta umowa też stronę czeską zobowiązuje do określonych informacji, które ma nam przekazywać, m.in. o wszystkich pozwoleniach wodnoprawnych, które w przypadku Uhelnej będą wydawane. Być może problem niedoboru wody wynika z nadmiernej eksploatacji przez podmioty gospodarcze po tamtej stronie. Na dzień dzisiejszy nie wiemy, jakie pozwolenia wodnoprawne są wydawane i jakie pozwolenia, na jaką ilość wody, na bieżąco wydaje strona czeska. Nie mamy też informacji na temat żwirowni. Żadna dyrektywa nie zobowiązuje do tak szczegółowego monitorowania i przekazywania informacji w obie strony. Dzięki temu my też będziemy mieli szczegółowe odczyty z monitoringu tych wszystkich parametrów, które będzie przygotowywała strona czeska, więc te informacje będą zobiektywizowane i oparte o uzgodniony system. Jeżeli chodzi o te inwestycje, rzeczywiście będzie dokończenie wału ziemnego i bariery ochronnej wód, drobna modernizacja oświetlenia, techniczny punkt pomiaru hałasu i stacje pomiaru jakości powietrza, otwory w warstwach wodonośnych celem pomiaru ilości i jakości wody. I te same inwestycje analogicznie po swojej stronie wykona strona czeska, żebyśmy mogli sobie te dane porównywać.

Na dzień dzisiejszy takich zasad polubownego rozstrzygania sporów między nami a Czechami w tej strefie przygranicznej, na obszarach górniczych, nie mieliśmy. W pierwszej kolejności powoływani są eksperci wewnętrzni delegowani przez strony, w drugiej kolejności eksperci zewnętrzni. Trzeci krok to pełnomocnicy, którzy na stałe zajmują się monitorowaniem tej umowy.

Trybunał orzeka wyłącznie w przedmiocie sporu, bez możliwości nakładania kar.

Bardzo proszę, pan poseł Marek Sawicki. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Chciałem na początku podziękować.

W wypowiedzi publicznej wiceminister Ozdoba mówił, że winę za nałożone kary ponosi minister Szymański, bo prawdopodobnie przedstawiciel Polski w Trybunale Sprawiedliwości nie był należycie przygotowany do przeprowadzenia obrony polskiego interesu, a w komunikacie Trybunału Sprawiedliwości mamy pełną informację, że strona polska nie wykazała, w jakim stopniu zamknięcie tej elektrowni grozi niedoborem energetycznym czy problemem energetycznym Polski. Nie zamknięto.

Bardzo proszę, pani minister. Dziękuję za to dobre słowo, ale nie do końca tak jest. Żeby ta umowa końcowo powstała, musiały pracować wszystkie resorty i eksperci. Mamy tak szczegółowo określone normy monitorowania, bo angażowały się w to GIOŚ, RDOŚ i wszystkie służby środowiskowe i geologiczne. Czas na wynegocjowanie tak szczegółowej i tak precyzyjnej umowy, żeby żadna ze stron nie mogła w przyszłości jej dowolnie interpretować, był niezbędny.

Natomiast w zetknięciu ze stroną czeską i rządem premiera Babisza potwierdzam to, co było wcześniej też komunikowane ze strony i ministra Kurtyki, i pozostałych uczestników tego dialogu: to nie był dialog. Wtedy były wybory, potem było po wyborach, formował się nowy rząd. Być może ten temat z jakichś względów był tematem potrzebnym w kampanii i podgrzewał spór polsko-czeski. Poza kurtuazyjnymi odpowiedziami nie byliśmy w stanie wrócić do rozmów merytorycznych. Nie było dobrej woli, nie było też chęci, żeby skupić się na szczegółach i rozmawiać o szczegółach. Jeżeli chodzi o Polskę i reprezentowanie nas przed Trybunałem, przypomnę tylko, że tam nie było czasu na dostarczenie jakiejś dużej ilości materiałów czy przedstawienie naszego stanowiska.

Nie mieliśmy informacji, że są jakiekolwiek wątpliwości co do tego. Przypomnę, że jak mamy naruszenie w związku z jakąkolwiek dyrektywą, bo te naruszenia czy dochodzenia w zakresie naruszeń się pojawiają, to najpierw Komisja pyta, potem są spotkania, setki listów, jakiś okres na ewentualne naprawienie i dopiero po jakimś czasie, często 2-3-letnim, pojawia się ewentualne orzeczenie. Natomiast wiemy, że trwa on bardzo długo.

Patrząc na elastyczność Trybunału i możliwość nałożenia kary finansowej jako środka tymczasowego, którego nałożenia traktat nie umożliwia (Dzwonek), wydaje się, że elastyczność w tej sytuacji jest też możliwa. Taki wniosek złożyliśmy z powołaniem się na konkretną podstawę prawną regulaminu, który ze względu na zmianę okoliczności pozwala karę wycofać. Mamy nadzieję, że ten wniosek będzie uwzględniony. Posłowie Joanna Borowiak i Lidia Burzyńska zadadzą pytanie w sprawie wysokości rządowego wsparcia dla jednostek OSP w zakupie wozów ratowniczo-gaśniczych na przestrzeni lat 2016-2022. Odpowie sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pan minister Maciek, przepraszam, Maciej Wąsik. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Jednostki ochotniczej straży pożarnej zajmują niezwykle ważne miejsce w polskim systemie ochrony przeciwpożarowej i w systemie ratowniczo-gaśniczym. Strażacy OSP w lokalnych społecznościach nazywani są cichymi bohaterami dnia codziennego. Dzięki swojej gotowości do bezinteresownego niesienia pomocy drugiemu człowiekowi są doceniani przez społeczeństwo. Służba druhów strażaków nie jest łatwa. Do ich codziennych zadań bowiem nie należy tylko gaszenie pożarów, ale również ratowanie ofiar wypadków drogowych czy pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Wyjątkową pomoc druhowie OSP kierują w sytuacji pandemii koronawirusa szczególnie do seniorów, niosąc im wsparcie w codziennych sprawach i potrzebach i pomagając w dotarciu do punktów szczepień przeciw COVID-19. Oprócz niesienia pomocy w chwilach zagrożenia dla lokalnych społeczności druhowie OSP są także doskonałymi przekazicielami polskich tradycji i wartości. Swoją pasją zarażają młodsze pokolenie, organizując i szkoląc dziecięce i młodzieżowe drużyny pożarnicze, dzięki czemu przekazywana jest misja niesienia pomocy często z narażeniem własnego zdrowia i życia. Zgodnie z dewizą: Bogu na chwałę, ludziom na pożytek druhny i druhowie OSP są obecni zawsze we właściwym miejscu o właściwym czasie. Rolę, jaką pełnią jednostki ochotniczej straży pożarnej w Polsce, docenia rząd Prawa i Sprawiedliwości, czego przykładem jest wsparcie finansowe oraz rzeczowe udzielane druhom ochotnikom na terenie całego kraju na skalę dotąd nieporównywalną. Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie: Ile samochodów zostało zakupionych w latach 2016-2022 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych? Jakiego typu i rodzaju były to wozy? W jakiej wysokości środki finansowe zostały na ten cel przeznaczone ogółem, z podziałem na województwa, w szczególności z uwzględnieniem województw kujawsko-pomorskiego, śląskiego, łódzkiego, mazowieckiego i podkarpackiego? Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Duża część naszego bezpieczeństwa to są ochotnicze straże pożarne, krajowy system ratowniczo-gaśniczy. Ten system, który jest unikalny na świecie, oparty na wolontariacie, na ochotniczej służbie, trzeba wspierać i rząd ten system wspiera. W latach 2016-2021 łącznie do jednostek OSP trafiło 2420 pojazdów specjalistycznych przeznaczonych do działań ratowniczo-gaśniczych.

Jak to się przedstawia w poszczególnych latach?

Te pieniądze nie przepadną, przejdą na następny rok, razem ze środkami przeznaczonymi w budżecie i nie tylko w budżecie, bo to są środki z narodowego funduszu ochrony środowiska, środki z firm ubezpieczeniowych, środki z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i oczywiście budżetowe środki MSWiA. W tym roku powinno być 518 samochodów zakupionych przez ochotnicze straże pożarne z kapitalną dotacją ze środków budżetu państwa.

Decyzją siedzącego tutaj komendanta głównego Straży Pożarnej zmieniono sposób użytkowania samochodów w Państwowej Straży Pożarnej, skrócono okres ich użytkowania, tak żeby w PSP były samochody jak najbardziej nowoczesne.

Chciałbym także zapewnić, że oprócz ustawy o ochotniczych strażach pożarnych rząd planuje i niedługo przedstawi Wysokiej Izbie następne pomysły dotyczące rozbudowy tego systemu. Dziękuję serdecznie. Witam pana serdecznie. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie Ministrze! Dziękuję panu ministrowi za tak merytoryczną i dającą radość informację, jeżeli chodzi o wspieranie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości ochotniczych straży pożarnych. Ta wypowiedź była możliwa ze względu na realne działania w okresie od 2016 r. do 2022 r. Ochotnicze straże pożarne to jednostki realizujące zadania w zakresie nie tylko ochrony życia, zdrowia, mienia, ale również zagrożeń ekologicznych w różnych miejscach.

Panie Ministrze!

Jakie plany w zakresie wsparcia dla ochotniczych straży pożarnych przewiduje się w przyszłych latach? Dziękuję. Bardzo proszę, panie ministrze. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Takie działania będziemy wspierać. Ale chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Nie chciałbym za bardzo wybiegać w przyszłość, ale myślę, że niebawem Wysoka Izba będzie mogła pracować - będzie to dla mnie ogromna przyjemność, jeżeli będę mógł prowadzić tę ustawę - nad nową ustawą, która poszerzy także zakres działania ochotniczych straży pożarnych. Będzie to ustawa, która troszeczkę zmieni system zarządzania kryzysowego.

Ten system będziemy starali się bardzo mocno rozbudowywać, żeby we wszystkich służbach liczba ratowników medycznych była jak najwyższa.

Myślę, że na wiele pytań pani poseł odpowiada ustawa o ochotniczych strażach pożarnych, która mówi o zapewnieniu całego cyklu szkoleń dla ochotników przez Państwową Straż Pożarną, gdzie mówimy, że wykształcenie ochotnika zdolnego do działań ratowniczych jest równoważne z wykształceniem strażaka zawodowego. Uważamy, że to jest dobra droga, że to jest właściwy kierunek, i chcemy w ten sposób rozwijać straże pożarne. To są także kursy, które już niebawem ruszą w Państwowej Straży Pożarnej dla kierowców kategorii C, dla młodych strażaków, którzy dopiero wchodzą w to swoje życie ratownicze, po to żeby mogli zastępować starsze pokolenia strażaków, którzy dotychczas prowadzili samochody strażackie, tak żeby ci młodzi mogli nie za swoje pieniądze, ale za środki zapewnione przez rząd zdobyć nowe kompetencje, żeby prowadzić działania ratownicze. Dziękuję panu komendantowi. Przechodzimy do następnego pytania. Posłanki Urszula Zielińska oraz Mirosława Nykiel zadadzą pytanie w sprawie ogólnopolskiej, antyunijnej kampanii Polskich Elektrowni - inicjatywy kontrolowanych przez Skarb Państwa wytwórców energii elektrycznej. Odpowie podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pan minister Karol Rabenda. Bardzo proszę panią posłankę Małgorzatę Tracz o zabranie głosu. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Od kilku tygodni jesteśmy świadkami pierwszej od czasów wstąpienia Polski do Unii Europejskiej otwarcie antyunijnej kampanii w przestrzeni publicznej. Na ulicach polskich miast, w radiu, w telewizji, w Internecie, w prasie, a nawet na naszych skrzynkach mailowych widzimy polexitową reklamę finansowaną przez spółki Skarbu Państwa, bo przecież za tą kampanią stoją Polskie Elektrownie, czyli Tauron, Enea, PGE, PGNiG. Ta antyunijna kampania wejdzie do kanonu przykładów kłamstw i manipulacji, bo to jest manipulacja, która ma wmówić ludziom, że 60% ceny na ich rachunkach za prąd to jest wina polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

Czy minister Sasin wiedział o tej planowanej kampanii? Być może ją opiniował czy zatwierdzał.

Zapraszam pana ministra. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Najwięksi krajowi wytwórcy energii: Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Połaniec, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz PGNiG Termika zainicjowały kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą kosztów produkcji energii elektrycznej. Kampania jest realizowana przez Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, które skupia producentów energii i w swojej kampanii odwołuje się właśnie do kosztów produkcji.

To nie są dane wzięte z kosmosu. To są bezsprzeczne dane, to są dane powszechnie dostępne, potwierdzone przez ekspertów. Bezsprzecznie wiadomo, że unijna polityka klimatyczna jest podstawową przyczyną podwyżek cen prądu. Jeszcze w 2016 r. cena uprawnień wynosiła 6 euro. Obecnie sięga 90 euro za tonę. Polska energetyka zmienia się, ale transformacja energetyczna to proces.

W związku z prawnym obowiązkiem spółki obrotu energią na przełomie lat 2021 i 2022 przekazały odbiorcom informacje w zakresie struktury kosztów sprzedawcy energii elektrycznej.

Reasumując, kampania ma charakter edukacyjno-informacyjny. Powstała z inicjatywy wytwórców energii, nie z inicjatywy rządowej. Wszelkie pytania dotyczące kampanii powinny zatem być kierowane do zarządów tych spółek, które są odpowiedzialne za prowadzenie bieżących spraw tych podmiotów. To są kampanie podmiotów wytwarzających prąd w Polsce, dostarczających ten prąd Polakom.

Dziękuję bardzo. Pani poseł Lidia Burzyńska. Bardzo proszę. Przepraszam za pomyłkę. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Chciałabym pokazać obrazek z 2016 r. z Wielkiej Brytanii. Kilka miesięcy później Brytyjczycy zagłosowali za brexitem. Szanowni państwo, to drugi obrazek. Na bilbordach są kłamliwie wygłaszane tezy, że za 60% cen energii odpowiada Unia Europejska. Te dwa obrazki, Wysoka Izbo, łączą dwie sprawy: kłamstwa i chęć przerzucenia nieudolności, zaniechań rządu w zakresie polityki energetycznej na Unię Europejską. Panie Ministrze!

Pan mówił, że to jest 60%, a wszyscy eksperci na rynku mówią, że to jest 20%. Odpowiedzcie Polakom, dlaczego się tak upieracie i chcecie wyprowadzić Polskę z Unii. PiS to polexit, ale Polki i Polacy doskonale wiedzą, jaką wartością jest Unia Europejska, i nie pozwolą na wyprowadzenie Polski z Unii.

Oczywiście bardzo chętnie na nie odpowiemy. Chciałem sprostować: to nie jest żadna kampania oszczerstw. To jest kampania informacyjno-edukacyjna. I nie będzie tak, że będziecie bronić tych decyzji Unii Europejskiej i przerzucać to na podmioty, które dostarczają prąd Polakom, w Polsce. Przechodzimy do następnego pytania. Pan poseł Marek Polak oraz pani poseł Barbara Dziuk - witamy w dobrym zdrowiu, pani poseł - zadadzą pytanie w sprawie zmiany systemu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Pytanie jest skierowane do prezesa Rady Ministrów, a odpowie, z upoważnienia prezesa Rady Ministrów, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pan minister Janusz Cieszyński. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie!

W tym czasie w czterech etapach w całej Polsce będą wyłączane stare nadajniki, a w ich miejsce włączane będą nowe. Na skutek tej zmiany część gospodarstw domowych może utracić dostęp do naziemnej telewizji cyfrowej, gdyż starsze telewizory nie obsługują nowego standardu i wymagają uzupełnienia w odpowiedni dekoder. W związku z tym, aby zminimalizować koszty tych zmian, przygotowywany jest program mający na celu dofinansowanie zakupu wspomnianego urządzenia. Chciałbym zapytać pana ministra, jaka jest skala gospodarstw domowych, które będą zagrożone utratą dostępu do telewizji naziemnej i czy program ma szansę zostać wdrożony przed pierwszym etapem zmiany sygnału, tj. przed 28 marca br. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kontynuuje pytanie pani poseł Barbara Dziuk. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Nowy standard oznacza techniczne zmiany dotyczące transmisji sygnału.

Jak to będzie wyglądać od strony technicznej? Czy problemy związane z tym przejściem będą w jakiś sposób poruszane w kampanii informacyjnej?

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie ministrze. Drugi dzień mam przyjemność prowadzić obrady, kiedy pan walczy z tematem. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! To też dla mnie wielka przyjemność mieć pana marszałka za plecami.

Dla każdego obywatela będzie dostępne dofinansowanie, dla każdego gospodarstwa domowego to dofinansowanie wynosi 100 zł.

Zgodnie z szacunkami Krajowego Instytutu Mediów, czyli jednostki, która podlega Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, takich gospodarstw domowych jest obecnie 2270 tys. Oczywiście te działania są już od jakiegoś czasu prowadzone we współpracy ze wszystkimi przedstawicielami mediów, bo jest to wspólny interes wszystkich mediów i wszystkich obywateli, żeby ta transformacja przebiegła sprawnie i szybko. Mamy informacje o tym, że prawdopodobnie obecnie ta liczba może być mniejsza, natomiast to są dane aktualne na moment przygotowania raportu, który ukazał się w ubiegłym roku. Jeżeli chodzi o kwestie związane z kampanią i z gotowością systemu, to ten projekt jest procedowany jako pilny.

Myślimy, że tak naprawdę już na początku marca będzie można pobierać bony i będzie można robić zakupy.

Tam ta zmiana wydarzy się jako pierwsza i stopniowo będzie to się przesuwało na wschód, a w końcu obejmie całą Polskę. Proces ten zakończy się pod koniec czerwca tego roku. Będzie prosty mechanizm, bon będzie można uzyskać przez e-usługę albo w placówkach Poczty Polskiej. Jeżeli chodzi o kampanię informacyjną, to jednym z elementów tej ustawy jest zapewnienie środków na kampanię. Ta kampania, mam nadzieję, będzie bardzo szeroka.

Z tego miejsca kieruję też wielki apel do wszystkich państwa parlamentarzystów: zaangażujmy się w to wspólnie, informujmy naszych czy państwa wyborców o tym, że taka zmiana nadchodzi, i w jaki sposób możemy do tego się przygotować. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z posiadanych informacji wynika, że zapowiadane zmiany nie będą dotyczyły abonentów telewizji kablowej i satelitarnej, gdyż cyfrowy tunel zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku nie jest wykorzystywany. Dziękuję. Dziękuję. Pani poseł, drugie pytanie. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zmiana sposobu nadawania nie powinna spowodować problemów w odbiorze.

Jak to technicznie będzie się odbywało?

Bardzo proszę, panie ministrze. Szanowny Panie Marszałku! Jeżeli chodzi o te pytania, to tak, potwierdzam, te zmiany nie obejmą innych technologii nadawania.

Dziękuję za pytania. Posłowie Mariusz Trepka i Andrzej Gawron zadadzą pytanie w sprawie projektu Narodowa Reprezentacja Akademicka. To pytanie posłowie zadadzą ministrowi edukacji i nauki, a odpowie sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki pan minister Włodzimierz Bernacki. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Narodowa Reprezentacja Akademicka - bardzo dobry projekt, trzeba go promować. W tej chwili już ruszyła trzecia edycja tego projektu dla studiujących sportowców. Chcemy mieć medale, w tej chwili trwają Igrzyska Olimpijskie. Osoby studiujące mogą z tego projektu skorzystać i chcemy, aby korzystały i promowały Polskę na arenie międzynarodowej. Dla tych, którzy realizują karierę sportową, przeznaczone jest dofinansowanie indywidualnych zajęć na uczelni. Wszystko po to, aby młodzi ludzie mogli równolegle uczyć się i rozwijać swoje talenty sportowe. Program organizuje ministerstwo edukacji we współpracy z Akademickim Związkiem Sportowym. Panie Ministrze! Jakie środki finansowe przeznaczone są na wsparcie edukacji studentów sportowców? Kto może uzyskać to wsparcie? Ilu studentów i z ilu uczelni wzięło udział w poprzednich dwóch edycjach tego projektu? Jakie kwoty wówczas przeznaczono na organizację dodatkowych zajęć? I jaki jest termin zgłoszeń do trzeciej edycji?

Dzięki takiemu właśnie wsparciu będzie to możliwe. Zapraszam, panie ministrze. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Nie tak dawno, właściwie w roku ubiegłym uczestniczyliśmy wszyscy w tym święcie sportu, jakim była olimpiada.

Te wspaniałe wyniki, które osiągają w sporcie, są następstwem ich aktywności, której my na co dzień nie widzimy.

To są ludzie, którzy mają rodziny, to są ludzie, którzy również bardzo często są studentami. 25% naszych olimpijczyków to członkowie akademickich zespołów sportowych, a więc studenci. Stąd też inicjatywa programu sportowego, o który pan poseł pyta, programu, który realizowany jest.

Warunek jest jeden: uczelnia musi spełniać wymogi dotyczące liczby studentów.

Tutaj na każdego studenta przewidziana jest kwota 18 tys. plus koszty pośrednie w wysokości 10%, czyli w sumie będzie dawało nam to prawie 20 tys. Jest to przeznaczone tak naprawdę na realizację 100 godzin dydaktycznych dla tych studentów, którzy ze względu na treningi, na uczestnictwo w zawodach sportowych nie mogą w normalnym trybie realizować swoich studiów, czy to studiów pierwszego, czy drugiego stopnia. Zatem te zajęcia, te godziny, które są przewidziane dla studenta olimpijczyka, to są zajęcia, które rzeczywiście mogą być realizowane najczęściej w trybie indywidualnym, ale też mogą być realizowane w trybie grupowym.

Pamiętajmy też, że w tym obecnym systemie rok akademicki nie pokrywa się z kolejnym rokiem studiów czy z rokiem kalendarzowym, ale tutaj dyscyplina budżetowa powoduje, że rozliczamy to rok po roku.

Dodam, że my rozliczamy (Dzwonek) faktycznie zrealizowane godziny.

Pan poseł Andrzej Gawron. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Dziękuję, panie ministrze, za tak szczegółowe informacje. Na pewno wsparcie studentów sportowców jest bardzo ważne, tym bardziej że w obecnym czasie, żeby osiągać wyniki, to musimy rzeczywiście mieć takie zaplecze, które pozwoli na to, żeby te wyniki osiągać. Mam takie pytanie. Były 3 mln wykorzystane, teraz prawie 9 mln. A jeszcze takie pytanie dodatkowe.

Dziękuję. Bardzo proszę, panie ministrze. Jeśli chodzi o dynamikę, to tak jak powiedziałem, jesteśmy w trakcie rozliczania tej drugiej edycji, a więc ta kwota była przyznana na poziomie.

Otóż te środki przeznaczone są przede wszystkim na to, co związane jest z dydaktyką. Pamiętajmy, że głównie są to studenci Akademii Wychowania Fizycznego, ale nie tylko. W związku z tym te środki przeznaczane są na realizację tych zobowiązań, które studenci przyjęli, rozpoczynając dany rok akademicki. Przypomnę, że te zobowiązania odnoszą się do liczby nie tylko ćwiczeń i wykładów, ale uzyskanych punktów ECTS. I w związku z tym, jeszcze raz powtarzam, chcemy przez ten rodzaj wsparcia, i mówimy tu tylko o jednym bardzo konkretnym programie, ułatwić i zabezpieczyć tym studentom możliwość ukończenia studiów w normalnym, właściwym terminie. Oprócz tego państwo mają świadomość tego, że akademickie związki sportowe uzyskują wsparcie zarówno ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki, ale również wielkich firm, koncernów, spółek Skarbu Państwa.

Ten pieniądz nie trafia indywidualnie do kieszeni studenta, to są środki przeznaczone dla uczelni, dla organizacji programu studiów. Dziękuję bardzo państwu. Przechodzimy do następnego pytania. Posłowie Fryderyk Kapinos i Kazimierz Gołojuch zadadzą pytanie w sprawie zwycięstwa w unijnym konkursie twinningowym dla Serbii konsorcjum instytucji rolniczych z Polski, Litwy i Francji. Na to pytanie odpowie sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan minister Ryszard Bartosik. Bardzo proszę pana posła Fryderyka Kapinosa o zadanie pytania. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pod koniec stycznia br. pojawiła się informacja o wygraniu przez konsorcjum instytucji rolniczych z Polski, Litwy i Francji unijnego konkursu twinningowego dla Serbii. Nasza Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest liderem tego konsorcjum. Od wielu lat Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako największa agencja płatnicza dla wspólnej polityki rolnej w Europie współpracuje ze swoimi odpowiednikami w wielu państwach członkowskich. Od kilku lat ARiMR brała aktywny udział w przekazywaniu doświadczeń z wdrażania instrumentów polityki rolnej, które wykorzystywane były m.in. w projektach realizowanych w Chorwacji, Mołdawii czy Azerbejdżanie. Po raz pierwszy ARiMR jest liderem takiego projektu. Jest to niewątpliwie sukces polskiej agencji płatniczej, na który od wielu lat pracuje poprzez szereg inicjatyw o charakterze międzynarodowym, organizując konferencje i warsztaty. Polska jest postrzegana jako lider procesu transformacji, który dobrze wykorzystał czas i środki pochodzące z Unii Europejskiej na rzecz zmian w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W związku z tym chciałem zadać panu ministrowi następujące pytania. Jakie są założenia programu współpracy bliźniaczej dedykowanej Serbii oraz ile czasu potrwa realizacja tego projektu? Dziękuję. Proszę, panie ministrze.

Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z partnerami z Litwy i Francji będzie realizowała projekt, o którym pan poseł wspomniał w swoim pytaniu. Agencja jest liderem projektu w konsorcjum z rolniczymi instytucjami Litwy i Francji, wygrała rywalizację w unijnym konkursie twinningowym dla Serbii. Konkurentem było konsorcjum złożone z agencji płatniczych Austrii, Włoch i Węgier. Wysoka Izbo! Niedawno, nie tak dawno przecież to myśmy uczyli się wspólnej polityki rolnej. Dziś szczęśliwie się tak składa, że możemy swoimi doświadczeniami dzielić się z innymi, dlatego też Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanęła do konkursu, który wart jest 1,8 mln euro i będzie realizowany przez naszą agencję. Współpraca bliźniacza, twinningowa to program finansowany przez Komisję Europejską, dzięki któremu państwa kandydujące do Unii Europejskiej mogą otrzymać merytoryczną pomoc od krajów będących już członkami Unii Europejskiej. Projekty takie w głównej mierze realizowane są przez prowadzenie specjalistycznych szkoleń oraz wyjazdów studyjnych. To wielki sukces naszej agencji i pracowników, którzy przygotowywali się przez długi czas do tego projektu. 13 stycznia br. odbyły się przesłuchania przed przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz Serbii dwóch rywalizujących konsorcjów i jak już wcześniej powiedziałem, konsorcjum, którego liderem jest Polska, zwyciężyło w tym konkursie i program będzie prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z agencjami płatniczymi Francji i Litwy. W ramach projektu trwającego 2 lata Serbowie mają otrzymać kompleksową wiedzę o funkcjonowaniu rynków rolnych w Unii Europejskiej potrzebną do ich organizacji w Serbii, regulacji prawnych czy rozwiązań administracyjnych. Komisja Europejska przeznaczyła na to 1,8 mln euro. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na kwiecień br. Chcę przy okazji powiedzieć, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie po raz pierwszy uczestniczy w takim konkursie, bo ma już doświadczenia w innych projektach.

Eksperci agencji brali również udział w projekcie na rzecz Rumunii.

Te moduły to: wzmocnienie sektora owoców i warzyw, wzmocnienie sektora wina, sektora produktów zwierzęcych, wzmocnienie zdolności administracyjnych w odniesieniu do sektora cukru, stworzenie warunków do sprawnego tworzenia i funkcjonowania (Dzwonek) organizacji producentów oraz stworzenie warunków do sprawnego tworzenia i funkcjonowania mechanizmów inwestycji rynkowych. Cieszę się, że nasza agencja może dzielić się swoimi doświadczeniami z Serbią, z krajem, który aspiruje do wejścia w struktury Unii Europejskiej. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Należy podkreślić, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest największą agencją płatniczą w Europie. Podejmuje wiele inicjatyw, przekazując swoje doświadczenia innym krajom. Dziękuję w tym miejscu kierownictwu i pracownikom Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za ogromne zaangażowanie na rzecz polskiego rolnictwa i doradztwa międzynarodowego.

I drugie pytanie: Jak zdaniem pana ministra powinna kształtować się współpraca (Dzwonek) na arenie międzynarodowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako lidera zmian w rolnictwie i na obszarach wiejskich w tej części Europy? Proszę, panie ministrze. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Tak więc była to bardzo dobra okazja i sposobność, aby przygotować się do prowadzenia projektu jako lider. Te doświadczenia bardzo nam się przydały.

Tak więc będziemy mogli się dzielić swoimi doświadczeniami. A mamy się czym dzielić, ponieważ wykorzystanie środków europejskich w rolnictwie, środków dystrybuowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jest na najwyższym poziomie - 100-procentowe.

Chcę podkreślić, że wygraliśmy ten projekt z drugim konsorcjum. Tamto konsorcjum miało już wcześniejsze, i to dużo, dużo większe, doświadczenia. Tak więc jest to ogromna szansa dla naszej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego pytania. Posłowie Krystyna Skowrońska i Krzysztof Piątkowski zadadzą pytanie w sprawie usunięcia ewidentnych błędów rządu dotyczących wypłaty dodatków osłonowych za wzrost cen energii elektrycznej i gazu. Na to pytanie odpowie podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pan minister Piotr Dziadzio. Bardzo proszę panią poseł Krystynę Skowrońską. Proszę bardzo. Dziękuję, panie marszałku.

Jakie to błędy? To są błędy organizacyjne. Nie przygotowano samorządów, nie rozmawiano z samorządami. Nie przekazano żadnych pieniędzy. Przecież państwo doskonale wiecie, że to jest przekroczenie przepisów ustawy o finansach publicznych. Dajcie i rozmawiajcie z samorządami o tych sprawach. Przecież dzisiaj samorządy, aby wypłacić takie dodatki osłonowe, muszą zgromadzić pełną dokumentację, bo są kryteria dochodowe, komu taki dodatek osłonowy można wypłacić. Bez zmian przepisów nie będzie szansy tego zrobić. Państwo po prostu musicie naprawić swoje błędy, usunąć te ewidentne błędy dotyczące wypłaty dodatków osłonowych. O to wnoszą samorządy. To, co państwo zaproponowali, 2% kwoty jako rekompensata za przeprowadzenie tej procedury, to jest zdaniem samorządów za mało. Terminy, które wskazaliście, są zdaniem samorządów za krótkie. Postulat, aby nie wypłacać w dwóch ratach, ale może w jednej racie, to postulat mieszkańców. A zatem pytanie: Kiedy wreszcie będziecie rzetelnie rozmawiać z samorządami i kiedy usuniecie państwo te błędy, o których mówią samorządy, tak aby mogły w okresie drożyzny, wysokiej inflacji wypłacić dodatki, które przygotowaliście? Tak jak Polski Ład był bublem i miał błędy, tak i to rozwiązanie jest niepozbawione szeregu błędów. Czekamy na naprawę. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, zapraszam i witam jednocześnie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo Posłowie! Krótko będę chciał ustosunkować się do zarzutów, które padły z ust pani poseł w zakresie dodatku osłonowego i realizacji wypłat.

Jest to najwyższe dotychczas wsparcie, którego udzielamy bezpośrednio osobom, które mogą być dotknięte problemem drożyzny. Dobrze, już powiem.

Jeśli chodzi o zainteresowanie, jest bardzo duże zainteresowanie tym dodatkiem, jak pani poseł zapewne wie. Z punktu widzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jak powiedziałem, ustawa została właściwie przygotowana, do tego zostały już wdrożone również dwa rozporządzenia, które funkcjonują, które realnie określają warunki przyznawania dodatku i procedury w tym zakresie.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, żeby rozwiać wszystkie te wątpliwości, stworzyło poradnik dla gmin, w którym wszystkie te kwestie zostały opisane i scharakteryzowane. Uważamy, że ten akt, który został wprowadzony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, jest absolutnie wykonalny. Wszystkie terminy są zgrane i wojewodowie w koordynacji z samorządami wypłacają środki.

To jest tylko kwestia, mówiąc otwarcie, dobrej organizacji, sprawnej organizacji i efektywnego wypłacania tych dodatków, o których mówimy, tak ażeby obywatele mogli szybko z tego skorzystać.

Nie widzimy tu żadnych problemów, to są kwestie organizacyjne. Według nas projekt jest przygotowany właściwie i spełnia też oczekiwania społeczne. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pytanie uzupełniające. Biorąc pod uwagę spektakularne fiasko waszego sztandarowego bubla legislacyjnego, jakim okazał się Polski Ład, trudno było oczekiwać, że napiszecie taki prosty projekt bez błędów - projekt wsparcia antyinflacyjnego dla najuboższych mieszkańców naszego kraju. Pominę oczywiste kwestie, takie jak trudności obywateli ze zrozumieniem i wypełnieniem 12 stron wniosku. Pominę fakt, że o przyznaniu dodatków w przypadku wniosków złożonych przed końcem sierpnia ma decydować dochód sprzed 2 lat. Mam jednak pytanie dotyczące uzupełnienia - mówiła też pani poseł o tym. Powierzyliście państwo zadanie obsługi wniosków samorządom, a nie wyposażyliście ich w odpowiednie środki finansowe i prawne. Grono potencjalnych beneficjentów jest bardzo duże, mówił pan minister o tym, to 7 mln gospodarstw. Czy rząd zamierza (Dzwonek) spełnić postulaty samorządowców i jednak naprawić ten bubel legislacyjny, czy, tak jak zrozumiałem z wypowiedzi pana ministra, nie zamierzacie państwo absolutnie robić nic? Bardzo prosiłbym o odpowiedzi na nasze pytania na piśmie. Również w tej sprawie złożona została interpelacja. Dziękuję bardzo. Odpowiada podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pan minister Piotr Dziadzio. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ja jeszcze raz, odpowiadając tutaj na wątpliwości, które zostały wskazane, powiem w ten sposób. Dla ułatwienia wypełnienia formularza, który naszym zdaniem jest prostym formularzem, nie jest trudnym formularzem, dodatkowo przygotowaliśmy materiał instruktażowy.

Jeśli chodzi o ułatwienia, oczywiście na każdym etapie, tam gdzie widzimy, że te ułatwienia są konieczne, wprowadzamy je.

Chodzi tutaj o Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków. Ale to w tym merytorycznym obszarze. Wydaje mi się, że odpowiedziałem panu posłowi na pytania. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Pytanie w sprawie negocjacji i porozumienia kończącego polsko-czeski spór o kopalnię Turów w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski, przygotowane przez posłów Prawa i Sprawiedliwości: panią poseł Barbarę Bartuś, panów posłów Grzegorza Lorka, Wojciecha Zubowskiego, Krzysztofa Tchórzewskiego, panią poseł Elżbietę Dudę i pana posła Marka Suskiego - skierowane do ministra klimatu i środowiska. Jako pierwsza pytanie zada pani poseł Barbara Bartuś. Uprzejmie proszę. Wysoka Izbo! Szanowna Pani Minister! Pytanie o kopalnię Turów i o porozumienie polsko-czeskie w ramach pytań bieżących dzisiaj pojawia się już drugi raz, bo to jest temat bardzo ważny. Cieszę się, że nawet opozycja uznała, że to porozumienie jest bardzo ważne, i cieszę się, że padły już w tej Izbie słowa uznania, że do tego porozumienia doszło, bo to jest bardzo ważne porozumienie. Pani Minister! Dziękuję za dotychczasową odpowiedź, którą słyszałam, a która w tej Izbie padła. Ale chciałabym jeszcze, żeby pani rozszerzyła swoją wypowiedź o określenie, na ile zwiększy się bezpieczeństwo energetyczne Polski po podpisaniu tego porozumienia, bo to porozumienie to nie tylko kwestia zakończenia sporu, tam jest wiele elementów. Jest też bardzo ważny drugi wątek - wątek pracowniczy. Przecież kopalnia i elektrownia zatrudniają wiele osób. Jak mówi pani europoseł Anna Zalewska, jest nawet 60 tys. osób zatrudnionych w kopalni, w elektrowni, w spółkach powiązanych. Wyobraźmy sobie, gdybyśmy wykonali zarządzenie TSUE i zamknęli tę kopalnię, ile osób mogłoby stracić pracę, ile należałoby wypłacić zasiłków dla bezrobotnych.

A więc na ten wątek pracowniczy, pani minister, gdyby pani zwróciła uwagę - jak ważne jest, że udało się to porozumienie podpisać, że kopalnia i elektrownia będą dalej pracować. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł. O udzielenie odpowiedzi uprzejmie proszę minister klimatu i środowiska panią Annę Moskwę. Jednocześnie przyłączam się do podziękowań kierowanych już przez panią poseł. Naprawdę, gratulacje, pani minister. Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! To jest nasz wspólny sukces i tak ten sukces trzeba traktować. Ja tylko w ostatnim momencie dopięłam kilka elementów, natomiast jest to sukces absolutnie całego rządu i całego zespołu Zjednoczonej Prawicy, i co do tego nie mamy wątpliwości. Nawet patrząc na proces powstawania tej umowy i ilość szczegółów, jakie tam są zawarte - to była mozolna praca, wielomiesięczne wypracowywanie szczegółowych elementów tej umowy. Trudno sobie wyobrazić, co by się wydarzyło, gdyby kopalnia była zamknięta. Takiego scenariusza nigdy nie było. W naszych dokumentach takiego scenariusza nie mamy, ponieważ nigdy tego w sposób poważny czy w jakikolwiek inny nie rozważaliśmy. Prawdopodobnie też gdyby zapytać moją czeską koleżankę, a wcześniej czeskiego kolegę, ministra środowiska, czy by taką decyzję w swoim państwie wykonali. Jestem przekonana, że żaden odpowiedzialny polityk, minister, premier takiej decyzji by nie wykonał. W przypadku Polski ta kopalnia to jest do 7% naszego bezpieczeństwa energetycznego. To jest bezpieczeństwo sieci nie tylko w tamtym regionie, ale w całej Polsce. Szkoda, że się nie stała jedna rzecz, że żaden z tych polityków nie pojechał do kopalni, do elektrowni, nie stanął twarzą w twarz przed tymi wszystkimi ludźmi, którzy tam pracują - tam jest zatrudnionych 5 tys. ludzi bezpośrednio, 60 tys. osób w podmiotach zaangażowanych w świadczenie usług w tym całym łańcuchu dostaw, żeby kopalnia i elektrownia funkcjonowały - i nie powiedział: Proszę państwa, proszę się pakować, nie będzie za chwilę prądu, nie będzie w domu ogrzewania, zamkniemy szpitale, respiratory, nic nie będzie funkcjonować, nie wiem, co mam zrobić, może się wyprowadźcie, może jakiś jeszcze inny scenariusz. Jest takie wyobrażenie, że kopalnię można tak jak telewizor pilotem, pyk, pyk, wcisnąć, włączyć i wyłączyć. Każda kopalnia w swojej decyzji środowiskowej, koncesyjnej ma cały plan zamykania kopalni, z poszanowaniem środowiska, z poszanowaniem zasobów wodnych. Ta kopalnia taki plan też ma, jak każdy inny podmiot górniczy, który w Polsce i na świecie funkcjonuje. A więc tutaj celem prawdopodobnym - bo też trudno ocenić z perspektywy racjonalności tego celu, ale tak jest w uzasadnieniu - był ten cel środowiskowy. Na pewno wykonanie tej decyzji poza katastrofalnym i nieakceptowalnym efektem społecznym wywołałoby katastrofalny efekt środowiskowy.

Na dzień dzisiejszy mamy wycofaną skargę i zażegnany spór, nie tylko tymczasowo. Wcześniejsze propozycje Czechów były takie: zapłaćcie, na chwilę obecną zamykamy spór. Ta umowa jest na tyle szczegółowa co do parametrów monitoringu, co do sposobu realizacji inwestycji, co do zaangażowania strony polskiej po stronie czeskiej i strony czeskiej po stronie polskiej przy wykonywaniu tych inwestycji, że nie pozostawia elementów niejednoznacznych, niedogadanych, wątpliwych, potencjalnie rodzących spór w przyszłości. Co więcej, umowa sankcjonuje sposób rozwiązywania sporów.

W pierwszej kolejności musi być wykorzystany poziom ekspertów skierowanych przez strony. Cały czas działa komisja transformacji transgranicznej. W skład tej komisji wchodzą przedstawiciele samorządów na poziomie województwa, powiatów i gmin. Końcowo, jeżeli nadal któraś ze stron uważa, że w przedmiocie tej umowy coś nie zostało wykonane.

Dziękuję bardzo, pani minister. Z pytaniem uzupełniającym pan poseł Grzegorz Lorek. Bardzo proszę, panie pośle. Pani Minister! Wysoka Izbo!

Chciałbym powiedzieć Wysokiej Izbie, że miałem przyjemność pracować w Bogatyni. Znam wielu wspaniałych inżynierów, którzy tam pracują całe życie, ich oddanie i trud. Chciałem dodać, że w Bogatyni nie ma takiego zakładu pracy, nie ma nawet pośredniego zakładu pracy, więc zamknięcie elektrowni i kopalni to gigantyczny problem dla tego regionu. Chciałem zapytać, ile państwo polskie musiałoby zapłacić - mówię tutaj o kosztach związanych z energetyką - w przypadku wyłączenia elektrowni i natychmiastowego zamknięcia kopalni.

Dziękuję bardzo za to pytanie.

Nie da się z dnia na dzień zastąpić w pełni funkcjonującego organizmu, jakim jest kopalnia i elektrownia działające na potrzeby całego regionu, ale też całej Polski, czymś, co byłoby szybkim rozwiązaniem. Nie ma takiego OZE, nie ma takich źródeł konwencjonalnych, więc ten scenariusz z założenia był niewykonalny w każdym parametrze. Gdybyśmy mieli popatrzeć na potencjalne skutki społeczne, potencjalne skutki gospodarcze i utracone korzyści. Przypominam, że węgiel nadal stanowi 70% naszej podstawy energetycznej. Te potencjalne straty szacowaliśmy na 3 mld.

Oni opowiadali, jak wyglądała ich codzienność w trakcie trwania tego sporu.

Wnioski do komisji petycji o zamknięcie kopalni. Głosy opozycji: tak, trzeba zamknąć - jeszcze tej opozycji, która ma dobry kontakt z tymi, którzy wydają takie decyzje w instytucjach europejskich, więc jeżeli coś mówi, to z perspektywy społecznej jest myślenie: pewnie coś wiedzą, może będzie jakiś kolejny wyrok, może jakieś inne działania, które doprowadzą do zamknięcia kopalni. A więc z perspektywy pracujących tam osób, ich rodzin, całego otoczenia i społeczeństwa ta szkoda społeczna, tak naprawdę codziennie wyrażająca się. Patrząc też na nowe zatrudnienia, na motywację, na cały ten element psychologiczny, który w tym całym procesie, myślę, jest niezwykle ważny przy takiej liczbie osób, widać, że ten spór powodował bardzo dużą szkodę, niepotrzebną eskalację emocji i szkodę społeczną. Myślę, że tamto społeczeństwo ani Trybunałowi, ani Czechom tego nie zapomni, bo to jednak były tygodnie stresu i absolutnej niepewności. Co istotne, nasze zapewnienia cały czas były poważne: nie zapłacimy i nie zamkniemy.

Co jest jeszcze istotne w tych relacjach polsko-czeskich, jesteśmy teraz przed prezydencją czeską. Prezydencja ma bardzo istotną rolę. Turów na pewno nie jest najważniejszym tematem naszych relacji.

Pojawił się taki dosyć ciekawy tweet, bo tu są różne głosy, czy ta umowa jest zasadna. A więc pojawił się taki tweet: mówi Fiala do premiera Morawieckiego: słuchaj, przez 15 lat nie możemy wypowiedzieć tej umowy, na co premier Morawiecki mówi: nie, pięć i koniec, na co Fiala mówi: dobrze, niech będzie kompromis: pięć. A więc to pokazuje, że ta umowa jest bardzo dobrą umową dla strony polskiej, i jesteśmy dumni z podpisania tej umowy. Dziękuję bardzo, pani minister. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 12. porządku dziennego: Informacja bieżąca. Przypominam, że na obecnym posiedzeniu Sejmu zostanie rozpatrzona informacja w sprawie realizacji sztandarowych programów polityki prorodzinnej wprowadzonych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, jak np. ˝Rodzina 500+˝, ˝Za życiem˝, ˝Dobry start˝, ˝Mama 4+˝, dodatkowe świadczenie trzynasta emerytura, oraz nowego, realizowanego w ramach Polskiego Ładu świadczenia rodzinny kapitał opiekuńczy, o której przedstawienie wnosił Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Przypominam również, że przedstawienie uzasadnienia wniosku przez posła przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a udzielenie odpowiedzi przez przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 5 minut. Wystąpienia posłów w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 2 minuty. Na zakończenie dyskusji głos zabierają kolejno przedstawiciel wnioskodawców oraz przedstawiciel Rady Ministrów. Wystąpienie przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a wystąpienie przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 5 minut. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie wystąpienia przedstawiciela Rady Ministrów. Czas przeznaczony na rozpatrzenie punktu: Informacja bieżąca nie może być dłuższy niż 90 minut. Uprzejmie proszę o zabranie głosu przedstawiciela wnioskodawców panią poseł Joannę Borowiak. Bardzo proszę, pani poseł, zapraszam na mównicę. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Jednym z głównych filarów polityki rozwojowej każdego państwa powinna być polityka rodzinna i właśnie polityka wobec rodziny, wspieranie jej rozwoju, ochrona to znak firmowy Zjednoczonej Prawicy. Zanim Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, problemy polskich rodzin były zaniedbywane, szczególnie jeśli chodzi o wychowanie dzieci czy opiekę nad osobami starszymi. Polskim rodzinom żyło się trudniej, co działało na niekorzyść całego państwa. I nie wolno nam o tym dzisiaj zapominać. Dla Polaków dziś to oczywiste, że korzystają z programów kierowanych do rodzin. Takiej właśnie polityki rodzinnej oczekują Polacy: kompleksowej, czyli skupionej na wielu dziedzinach życia rodzinnego, i konsekwentnej, czyli żywo reagującej na aktualne problemy i potrzeby rodzin. Każdy kolejny program dla rodzin to sukces mierzony poziomem zadowolenia adresatów. Na stałe w pakiet prorodzinny wpisały się takie programy jak sztandarowy program ˝Rodzina 500+˝, który powstał po to, by wspierać polskie rodziny i zapewnić im stabilizację. Dla Prawa i Sprawiedliwości rodzina jest na pierwszym miejscu. Dzięki programowi ˝Rodzina 500+˝ polska bieda przestała mieć twarz dziecka, a jedną z największych hańb III RP - głodne dzieci - wysłaliśmy do historii. Do rodzin trafiło ponad 176 mld zł, dzięki którym rodzice z dziećmi mogą pozwolić sobie na wakacyjny wyjazd, zakup niezbędnego sprzętu lub potrzebnych artykułów czy wreszcie na drobne przyjemności, które kiedyś były poza ich zasięgiem. Kolejny program to ˝Dobry start˝, 300 zł wyprawki szkolnej, dzięki którym zakupy przyborów lub tornistra na nowy rok szkolny nie stanowią już wyzwania, a istniejące wcześniej nierówności pomiędzy uczniami zostały zniwelowane. Dzięki programowi ˝Mama 4+˝ realnie wspieramy osoby, które poświęcając się wychowaniu czwórki i więcej dzieci, nie zdołały wypracować sobie prawa do emerytury. Wcześniej nie miały one prawa do świadczeń i żyły na granicy ubóstwa. Polityka prorodzinna rządu Prawa i Sprawiedliwości to także wsparcie dla tych rodzin, które spodziewają się narodzin lub wychowują dzieci z niepełnosprawnościami. To dla nich stworzyliśmy program ˝Za życiem˝ z podwojonym finansowaniem na lata 2022-2026. Wspieramy rozwój instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi, pokazując, że można zrobić dużo więcej, niż zrobili nasi poprzednicy. Program ˝Maluch+˝ w 2015 r. to zaledwie 84 tys. miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Rodzina to też młodzi ludzie wchodzący w dorosłe życie i zaczynający swoją pracę zawodową. Dzięki programowi ˝Bez PIT dla młodych˝ mogą cieszyć się większą wypłatą i realizować nakreślone przez siebie plany. Rodzina to również seniorzy, którym poświęcamy wiele uwagi, bo wsparcie osób starszych jest niezwykle ważnym elementem polityki społecznej Prawa i Sprawiedliwości. Przywróciliśmy wcześniejszy wiek emerytalny, wydłużony przez Platformę i PSL, i skierowaliśmy do seniorów dodatkowe wsparcie finansowe. 36 mld zł w ubiegłym roku trafiło do portfeli seniorów. To 10 razy więcej, niż przeznaczył dla nich rząd Platformy i PSL-u w 2015 r. 35 mld dla blisko 10 mln emerytów w ramach ustawowo zagwarantowanej trzynastej emerytury i 46 mld zł wypłaty z trzynastej i czternastej emerytury łącznie. W 2015 r. zastaliśmy 99 domów seniora dla zaledwie 2800 osób. Dziś ponad 25 tys. seniorów ma do swojej dyspozycji ponad 1000 domów i klubów. Stworzyliśmy program ˝Opieka 75+˝ i ˝Leki 75+˝, a w czasie pandemii - ˝Solidarnościowy korpus wsparcia seniorów˝ Wychodzimy naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami. W odpowiedzi na aktualne potrzeby polskiego społeczeństwa rząd przygotował kolejne projekty, w tym rodzinny kapitał opiekuńczy oraz oczekiwaną przez seniorów emeryturę bez podatku.

Planowe w budżecie państwa wydatki na wsparcie rodzin i politykę społeczną w wysokości 112 mld zł w br. pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość jest gwarantem prowadzenia konsekwentnej i rozwojowej polityki prorodzinnej.

Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Przede wszystkim bardzo chciałabym podziękować za temat dzisiejszej informacji, tak ważny dla polskich rodzin i dla Polski. Dziękuję, że możemy porozmawiać o rodzinach i przede wszystkim podsumować ostatnie 6 lat. Od ponad 6 lat, wsłuchując się w potrzeby ludzi, konsekwentnie zmieniamy na lepsze wiele obszarów funkcjonowania państwa. Sprawne zarządzanie, w tym zmiany w systemie finansów publicznych, pozwoliło na wygospodarowanie środków finansowych, które stały się źródłem finansowania wielu programów społecznych, o których pani poseł już mówiła. Zmieniły się przede wszystkim warunki funkcjonowania społeczeństwa. Trudna sytuacja, z którą walczymy od 2 lat, czyli epidemia koronawirusa, nie spowolniła realizacji tych programów. Nie tylko utrzymaliśmy wszystkie rozpoczęte przed pandemią COVID-19 programy społeczne, lecz także rozwijamy je i wzbogacamy o kolejne instrumenty. Wszystko to pomimo olbrzymich wydatków związanych z koniecznością ochrony życia i zdrowia Polaków w obliczu epidemii, a także ratowania polskiej gospodarki przed głębokim kryzysem mogącym cofnąć rozwój Polski na dekady. W tych wyjątkowo trudnych warunkach realizowane przez nasz rząd programy społeczne stały się swoistymi tarczami antykryzysowymi wspierającymi tych, którzy bez interwencji państwa najprawdopodobniej nie poradziliby sobie sami albo też ich sytuacja uległaby radykalnemu pogorszeniu. Wypracowaliśmy mechanizmy wsparcia wielu grup społecznych: z jednej strony seniorów, z drugiej rodzin z dziećmi. Długofalowa, konsekwentna polityka prorodzinna jest przede wszystkim wyzwaniem.

Natomiast łączne wydatki na realizację polityki społecznej to blisko 112 mld zł. Szanowni Państwo! Wiele w przestrzeni publicznej mówimy na temat programu ˝Rodzina 500+˝ Przede wszystkim jest to program, który zmienił oblicze polskich rodzin. To potężne wsparcie, to inwestycja w rodzinę.

Program ten rozwijał się, ewoluował.

Twierdziła, że kobiety będą ubywały z rynku pracy, że przede wszystkim program jest źle przygotowany. Program przede wszystkim pokazał swoją skuteczność i zmienił oblicze polskiej rodziny, tak jak powiedziałam. Warto też spojrzeć na dane związane z rynkiem pracy i aktywnością kobiet na rynku pracy.

Program ˝Rodzina 500+˝, tak jak powiedziałam, ewoluuje. W tym roku wnioski składane są tylko drogą elektroniczną.

Są one składane o 50% szybciej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, a przejęcie obsługi tego świadczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli wymierne korzyści dla budżetu państwa, przekuły się w to, że mamy kolejny nowy program prorodzinny.

I tak jak powiedziałam, kolejne świadczenie. Przede wszystkim mamy przemyślaną politykę prorodzinną. Musimy wprowadzać instrumenty, które pozwolą nam wyjść z pułapki niskiej dzietności.

Kolejne wsparcie.

A więc przede wszystkim realizacja poprzez automatyzację, usprawnianie procesów. Również rozwiązanie ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym zakłada kolejne wsparcie dla rodzin.

Przez 6 lat sprawowania rządów przez Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczoną Prawicę ponad 2 mld zł zostało zainwestowane na utworzenie nowych miejsc. Kiedy w 2015 r. obejmowaliśmy rządy, było ok. 84 tys. Przede wszystkim zależy nam na tym, aby stworzyć warunki, aby samorządy, jeżeli jest taka potrzeba, w każdej gminie mogły otworzyć żłobek.

Tutaj mamy przywrócenie wieku emerytalnego, waloryzację świadczeń, trzynastą i czternastą emeryturę i zmiany, które są przygotowane w polityce podatkowej na ten rok.

Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze zapisać się do głosu? Zamykam listę. Ponieważ bardzo wiele osób zapisało się, a chciałabym każdemu umożliwić zabranie głosu, proszę o dyscyplinę.

Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Pani Minister! Szanowni Państwo! Wprowadzamy programy i w tym jesteśmy wiarygodni i konsekwentni. Nie będę tych wszystkich programów wymieniać, stąd pewnie tak długie było przemówienie pani minister, ponieważ nie sposób w ciągu 2 minut przedstawić całego dobra, które się zadziało, jeżeli chodzi o politykę prorodzinną za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Przedstawiliśmy, tak jak powiedziałam, optykę myślenia. Proponuję taki eksperyment, szanowni państwo. Nie ma tych wszystkich programów, nie ma ˝500+˝, nie ma ˝300+˝, nie ma ˝Dobrego startu˝ Emeryci za waszych rządów pracują za waloryzację, 3 zł, do śmierci, do 67. roku życia. Jakie jest użłobkowienie i jak wygląda ta polityka za waszych rządów? Jest też raport Najwyższej Izby Kontroli z 2015 r., który w sposób druzgocący ocenia waszą politykę.

Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Pani Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny! Niech pani przestanie kłamać. Do 2015 r., przez te 8 lat, wprowadziliśmy jeden z najdłuższych urlopów macierzyńskich, rodzicielskich w Europie. Po drugie, to my wprowadziliśmy darmowe podręczniki. Po trzecie, urlopy ojcowskie, to również my je wprowadziliśmy. Po czwarte, program ˝Maluch˝, czyli użłobkowienie, to program Platformy i PSL-u. Po czwarte, przedszkola za złotówkę. Ale to, co dzisiaj jest najbardziej interesujące i na czym nam zależy jako posłom opozycji, to żebyście państwo nie krzywdzili samotnych rodziców. Dla przykładu powiem państwu tak. Do pani minister się zwracam: Czy to jest prawda, czy nie?

To były ulgi prorodzinne, które wprowadził rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Pani Minister! Czy prawdą jest, że samotni rodzice w wyniku tego niby-ładu zostaną dzisiaj skrzywdzeni w ten sposób, że nie będą mogli odliczyć sobie przy średnich dochodach takiej ulgi, jaką będą mogły odliczać np. małżeństwa bezdzietne? Bo małżeństwa bezdzietne odliczą ponad 5 tys. zł (Dzwonek) przy średnich dochodach, a samotni rodzice - 1500 zł. Nie okradajcie samotnych rodziców. Przywróćcie im należne prawa, które mieli od 30 lat. Dziękuję, pani poseł. Bardzo proszę, pani poseł, o spokój, o zachowanie umiaru. Dajmy możliwość wypowiedzenia się. Każdy ma prawo zabrania głosu. Pan poseł Rafał Adamczyk, klub Lewica. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Nie będę pytał o czternastkę dla emerytów, bo jej nie ma w tym roku. Zapytam o program ˝Maluch+˝ Jest to inicjatywa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, która miała wspierać rozbudowę systemów opieki nad dziećmi do lat 3. Projekt ten miał ułatwiać powstawanie żłobków, klubów dziecięcych, a także zapewniać bardziej atrakcyjne warunki osobom samozatrudnionym, pracującym jako dzienny opiekun. W listopadzie tego roku niestety program nie został ogłoszony. Nie ma nowego naboru. Brak jest jakichkolwiek informacji na temat tego programu. Bardzo bym prosił o informację, kiedy zostanie on uruchomiony. Tutaj było zapewnienie pani minister, że będzie kontynuowany.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Mieczysław Kasprzak, Koalicja Polska. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Trzeba realnie patrzeć na to, co się robi.

Popatrzmy więc dzisiaj na ceny energii, na ceny towarów w sklepach. Nie poprawiła się demografia. Dzisiaj, przy tej drożyźnie - kogo stać na budowę mieszkania? Emeryci.

Bardzo proszę.

Bardzo proszę, panie pośle. Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Sytuacja osób niepełnosprawnych jest taka, że chce się wstać i zejść z tego wózka - mówi Łukasz Krasoń, ekspert ruchu Polska 2050 do spraw niepełnosprawności. Ale Łukasz nie zejdzie z wózka, dlatego że jedyną częścią ciała, nad którą ma władzę, jest prawa dłoń.

Te 2 tys. do każdego pełnego etatu z PFRON-u dzisiaj wystarczają na pokrycie ok. połowy kosztów zatrudnienia, a jeszcze kilka lat temu było to ponad 60%. Pomimo wzrostu płac ta kwota stoi w miejscu. Podobnie jest zresztą z wpływami na fundusz rehabilitacyjny w zakładach pracy chronionej. Nawet proste rzeczy są poza waszym zasięgiem. Wczoraj usiłowałem przekonać, że dofinansowanie do odbiorników nowej telewizji naziemnej powinno objąć także telewizory, dlatego że nowy standard niesie ze sobą całą masę ułatwień dla osób niedosłyszących albo niedowidzących. Bez efektu. Zapraszam, pani poseł. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Na początek bardzo chcę podziękować pani poseł Joannie Borowiak za to, że jest ta informacja bieżąca, dzisiaj możemy tutaj o tym rozmawiać. Dziękuję za tę szeroką wypowiedź, chociaż skróconą, pani minister, bo to jest temat bardzo obszerny i bardzo ważny, ważny dla Prawa i Sprawiedliwości, ale myślę, że ważny przede wszystkim dla Polski, dla polskich rodzin, a to jest nasza przyszłość. Pani minister mówiła o wielu programach, które zostały wprowadzone w ogóle po raz pierwszy do naszego systemu prawnego, do budżetu państwa, bo przecież jeżeli mówimy o 500+, to on jest w budżecie państwa w pozycjach bardzo wysokich, bo to są miliardy złotych, które płyną do polskich rodzin, ale nastąpiły w tym. Powstają nowe programy, ale ten nasz sztandarowy program 500+ zostaje od tego roku zmieniony: tylko wnioski przez Internet, będzie wypłacał ZUS, zatem zmniejszą się koszty obsługi, odpadną też dodatkowe dochody dla samorządów. Przy tej okazji zrodziło się wiele pytań. Były wielkie krzyki opozycji, że to się nie sprawdzi, że będą problemy ze złożeniem wniosku. Mam pytanie do pani minister, bo już skończył się styczeń, mamy luty, czyli to już zaczęło funkcjonować, tak jak ˝Dobry start˝ (Dzwonek) od tamtego roku. Czy faktycznie są problemy ze złożeniem wniosku do ZUS-u? Ile tych wniosków do tej pory wpłynęło? Pani poseł Monika Rosa, Koalicja Obywatelska. Pani Minister! Wysoka Izbo! Polska rodzina potrzebuje wsparcia nie tylko wtedy, kiedy jest idealna, ale przede wszystkim wtedy, kiedy coś dzieje się nie tak, kiedy pojawiają się dzieci z niepełnosprawnością, kiedy pojawia się kryzys w rodzinie, kiedy potrzeba jest po prostu realnego, systemowego wsparcia, nie tylko finansowego. Dlatego pytam o system pieczy zastępczej. Co udało się zrobić przez te ostatnie lata w ramach systemu pieczy zastępczej? Wciąż jest za mało rodzin zastępczych, wciąż małe dzieci, dopiero co urodzone, trafiają do instytucji, wciąż są domy instytucjonalnej opieki nad małymi dzieciaczkami, wciąż po kilkanaście miesięcy, a nawet kilka lat dzieci spędzają w zawieszeniu prawnym, ponieważ trwają procesy w sądach i nie wiadomo, do kogo trafi opieka rodzicielska. Chciałabym, aby systemem wsparcia otoczone były rodziny, w których występuje przemoc domowa, aby dzieciom wierzono i były natychmiast izolowane od oprawców i od przemocowców, aby na pierwszym miejscu stawiano dziecko, a nie integralność rodziny biologicznej, żeby to właśnie bezpieczeństwo dziecka było najważniejsze, żeby przemoc domowa była czymś, z czym państwo będą systemowo walczyć. Ale ustawa o przeciwdziałaniu przemocy wciąż nie jest nowelizowana, wciąż na tę nowelizację czekamy. Kontrola NIK pokazała, że program ˝Za życiem˝ jest realizowany w bardzo niewielkim stopniu. Wciąż brakuje asystentów społecznych, wciąż brakuje reformy systemu orzekania, wciąż nie ma programu deinstytucjonalizacji wdrażania - tych rzeczy po prostu brakuje. Pan poseł Jan Szopiński, klub Lewica. Pani Minister! Pani minister powiedziała tutaj o przemyślanej polityce prorodzinnej. W związku z powyższym chciałbym zadać trzy pytania. Pytanie pierwsze: Kiedy zostaną uruchomione środki w ramach programu ˝Maluch+˝, jakie będą te środki i czy miejsca, które powstały w ramach tego programu, będą mogły być również dofinansowane? Pytanie drugie. Emeryci uwierzyli panu prezesowi, że będzie czternastka. Nie po raz pierwszy dość naiwnie uwierzyli, ale mam pytanie: Czy będzie ta czternastka, czy może pani minister skontaktować się z panem prezesem, czy są prowadzone w tej sprawie jakieś prace? Mianowicie rodzice samotnie wychowujący dzieci skarżą się, że zmiany podatkowe wprowadzone od początku 2022 r. w ramach rządowego programu Polski Ład pozbawiły ich możliwości preferencyjnego opodatkowania. Rzecznik praw obywatelskich w piśmie do ministra finansów wyraził swój sprzeciw wobec możliwości wspólnego rocznego rozliczenia PIT. Pan rzecznik zaapelował do ministra finansów o zainicjowanie prac legislacyjnych w celu przywrócenia poprzedniej regulacji. Ponieważ pan minister się zwinął, to mam prośbę do pani minister, żeby pani minister ustaliła, czy te prace zostały zainicjowane. Dziękuję bardzo. Pan poseł Dariusz Klimczak, Koalicja Polska. Szanowna Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Niedawno została ogłoszona uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie tzw. programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ˝Za życiem˝ Pytanie zasadnicze brzmi: Dlaczego projekt tej nowelizacji nie był przekazany do konsultacji publicznych, w tym z osobami niepełnosprawnymi, co w opinii wielu ekspertów stanowi naruszenie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych? Brak tych konsultacji dziwi tym bardziej, że po 5 latach, w listopadzie 2021 r. kontrolerzy NIK nie zostawili suchej nitki na tym programie. W tej sytuacji wydawałoby się, że państwo skorzysta, odpowiedzialne państwo skorzysta z opinii obywateli. Myślę, że w tym względzie zgodzi się ze mną przesympatyczna pani przewodnicząca Urszula Rusecka, która w swoim wystąpieniu zwracała uwagę na wagę kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Najważniejsze pytanie emerytów w tym roku: Czy pani minister mogłaby podać datę, kiedy na konta emerytów wpłynie czternasta emerytura? Jeżeli pani wie, że nie wpłynie, to chciałbym usłyszeć odpowiedź dlaczego. Pewnie to interesuje bardzo wielu emerytów, którzy na was głosowali.